Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 39. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 43. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druki nr 793 i 800) Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoki Sejmie! W imieniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawiam sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, druki nr 793 i 800. Senat do przedłożenia sejmowego tej ustawy zgłosił dwie poprawki o charakterze legislacyjno-porządkującym przejrzystość zapisów tej ustawy. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druki nr 794 i 814) Proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, druk nr 794. Marszałek Sejmu zgodnie z art. 54 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 30 listopada 2020 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zebrała się na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020 r. Po rozpatrzeniu 10 poprawek komisja rekomenduje przyjęcie wszystkich poprawek.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem ww. poprawek, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, przeciw - 446, 1 się wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 3., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Nikt nie był za, przeciw - 452, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 6. i 8., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki 7., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Nikt nie był za, przeciw - 449, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druki nr 795 i 818) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z druków nr 818 i 795. Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w dniu 8 grudnia br. i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek zgłoszonych przez Senat. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

1 - za, przeciw - 452, 1 się wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 760-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Piotra Polaka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 720. Podczas drugiego czytania tutaj, w Izbie plenarnej, zostały zgłoszone cztery poprawki do tego projektu.

Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 2., zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 760, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 703. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 703, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 635-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Panie i Panowie Posłowie! W imieniu połączonych komisji: sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiam dodatkowe sprawozdanie połączonych komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej, druki sejmowe nr 240 i 630. W drugim czytaniu projektu powyższej ustawy została zgłoszona jedna poprawka dotycząca bardziej elastycznego przyznawania odpraw dla odchodzących z tych przedsiębiorstw dyrektorów. Połączone komisje po wysłuchaniu wnioskodawcy poprawki oraz strony rządowej i po przeprowadzeniu dyskusji rekomendują Wysokiej Izbie odrzucenie tej poprawki. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 635. Poprawka zgłoszona została do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 635, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 680, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia z druku nr 688. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 688, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 810. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 810, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 820. Komisja przedstawia wniosek mniejszości, nad którym głosować będziemy w pierwszej kolejności. We wniosku mniejszości do art. 1 projektu ustawy wnioskodawcy proponują skreślić pkt 3. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku mniejszości, zechce nacisnąć

Głosujemy nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 820, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 178, zechce nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek przyjął. Proszę państwa, na tym zakończyliśmy głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowania podmiotów leczniczych na zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19 oraz działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Proszę ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego o przedstawienie informacji. Zapraszam, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Dzisiaj chciałbym przedstawić informację opartą na faktach, informację o tym, jak wygląda przebieg pandemii, ale też jak wyglądają narzędzia i instrumenty walki z pandemią, jakie rząd pana premiera Morawieckiego zastosował, szczególnie w okresie od września br. Dyskusje dotyczące pandemii bardzo często niestety mieszają fakty z emocjami. Ci pseudoeksperci oczywiście wypełniają przestrzeń Internetu. Niestety prowadzi to do dezinformacji, prowadzi to do budowania lęków, budowania obaw, niepokoju i budowania postawy strachu.

Po pierwsze, tak jak cały świat, tak i Polskę dotknęła druga fala epidemii, której szczyt, jak państwo doskonale wiecie, przypadł na początek listopada. Ale pandemia zaczęła przyspieszać tak naprawdę już w połowie października i wtedy rozpoczął się proces gwałtownego rozwoju, gwałtownych przyrostów dziennej liczby zachorowań. Ta kumulacja, ta eskalacja nastąpiła na początku listopada. Potem pandemia zaczęła zwalniać - zwalniać i na poziomie dynamiki, i na poziomie samej liczby zachorowań, którą bardzo ściśle monitorowaliśmy, patrząc na to, jak z tygodnia na tydzień wygląda liczba zachorowań. Ten trend, który pojawił się od początku listopada, doprowadził do tego, że już pod koniec listopada mieliśmy dynamikę ujemną liczby zachorowań.

Przebieg epidemii był bardzo charakterystyczny. Ale ta fala może mieć różny kształt, w zależności od tego, jakie środki są przedsiębrane w związku z walką, bo ta fala może być spłaszczona, ta fala może trwać bardzo długo, ta fala może mieć niski szczyt, może mieć szczyt wysoki. Robiliśmy wszystko, żeby liczba zachorowań była jak najbardziej ograniczona. Przede wszystkim przygotowywaliśmy się do tej fali poprzez zarządzanie liczbą dostępnych łóżek i respiratorów.

Staraliśmy się cały czas pilnować tego, żeby przyrost hospitalizacji był mniejszy niż przyrost bazy łóżkowej przeznaczonej dla chorych na COVID. Nazwaliśmy sobie to buforem bezpieczeństwa, bo chcieliśmy, żeby zawsze była wolna przestrzeń, wolna liczba łóżek przeznaczonych na leczenie COVID w stosunku do liczby hospitalizacji. Ten proces oczywiście był skojarzony czy stowarzyszony z tym, jak rozwijała się pandemia. Od końca października do końca listopada podwoiliśmy liczbę łóżek przeznaczonych na leczenie COVID. W połowie października czy pod koniec października mieliśmy mniej więcej 20 tys. łóżek, które chcieliśmy właśnie przeznaczyć na system COVID-owy. Potem przetaczała się fala pandemii i ta liczba zachorowań rosła. Kumulacja, tak jak powiedziałem, była na początku listopada. Doszliśmy do tego, że liczba ogólna łóżek przeznaczonych na zachorowania COVID-owe w tym maksymalnym punkcie wyniosła 40 tys.

Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, kiedy karetka musiała jeździć od szpitala do szpitala, ale na te sytuacje również bardzo szybko staraliśmy się odpowiedzieć, wprowadzając specjalne rozwiązania informatyczne, angażując wojsko ochrony terytorialnej do tego, żeby informacja, która trafia do dyspozytorów karetek, była informacją prawdziwą, której nie muszą weryfikować na miejscu, tylko taką, która pozwoli zawieźć pacjenta, sprawnie przewieźć go do szpitala. Tutaj też pilnowaliśmy przez cały okres buforu bezpieczeństwa. W przypadku łóżek jesteśmy teraz już w takiej sytuacji, że w związku z malejącą liczbą zakażeń mamy troszeczkę mniejszą infrastrukturę przeznaczoną na COVID, bo tą infrastrukturą trzeba bardzo elastycznie zarządzać. Trzeba elastycznie zarządzać, ponieważ mamy inne choroby i one również są bardzo poważnym problemem zdrowotnym Polaków.

Zorganizowaliśmy cały system dystrybucji tlenu, tak żeby tlen trafiał do pacjentów, żeby nie było zagrożenia brakiem tlenem w przypadku tych pacjentów, którzy go intensywnie potrzebują. Tutaj działaliśmy razem z Ministerstwem Aktywów Państwowych i udało się doprowadzić do sytuacji, że lokalne zapasy czy lokalne magazyny wojewódzkie tlenu zaczęły regularnie nadążać za zapotrzebowaniem, które było zgłaszane przez szpitale. Oprócz tlenu krytycznym lekiem czy lekiem stosowanym w terapii jest Remdesivir.

To samo zresztą dotyczy osocza. Początkowo dostawy Remdesiviru do Polski były rzędu kilku tysięcy ampułek miesięcznie. Udało nam się tak przeformułować umowy, tak zwiększyć te dostawy, że zarówno w listopadzie, jak i w grudniu osiągnęliśmy poziom dostaw do Polski sięgający blisko 50 tys. ampułek miesięcznie, tak że tutaj sytuacja też jest zabezpieczona. Chodzi tu o obostrzenia i ten hamulec bezpieczeństwa, który nacisnęliśmy pod koniec listopada, wprowadzając te najbardziej dolegliwe obostrzenia, z którymi zresztą teraz mamy do czynienia. To zahamowało również wzrost zachorowań, bo zamknięcie szkół, przejście na zdalne nauczanie, ograniczenie handlu, ograniczenie również podróży - to wszystko przyczyniło się do tego, że mamy mniejszą liczbę zachorowań i możemy się w tej chwili z większym spokojem zapatrywać na przyszłość. Szanowni Państwo! To są oczywiście takie bardzo podstawowe, najważniejsze działania, jednak mamy dwa ważne zdarzenia, dwa ważne zjawiska, o których też trzeba powiedzieć. Po pierwsze, sytuacja jest rzeczywiście lepsza niż 3–4 tygodnie temu, ale to nie znaczy, że jesteśmy w pełni bezpieczni. Niestety widmo trzeciej fali cały czas wisi nad całym światem, nie tylko nad Polską, i to widmo w niektórych miejscach na świecie się materializuje. Materializuje się chociażby w Korei, w Japonii, gdzie ta trzecia fala wystąpiła.

powinny dać państwu do myślenia, szczególnie że tak często powołujecie się na swoich wyborców, powołujecie się na wyborców w swoich regionach. Bardzo proszę o wyświetlenie pierwszego slajdu. Kwestia zgonów, która do dzisiaj nie została wyjaśniona. Tylko w listopadzie mamy o 30 tys. więcej zgonów niż w roku 2019 czy w roku 2018. Panie ministrze, bardzo pana proszę o precyzyjną odpowiedź. Tylko 10 tys. zgonów to są zgony związane z COVID-em, 20 tys. przypadków śmierci to są zgony niewyjaśnione, co do których rząd w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, co się stało. Czy to jest załamanie systemu? Czy to są wszystkie historie takie, że do naszych bliskich nie przyjechały karetki? Czy to jest kwestia braku terapii onkologicznych? Czy to jest kwestia po prostu załamania całego systemu służby zdrowia? 20 tys. niewyjaśnionych przypadków śmierci to mniej więcej tyle co 100 katastrof lotniczych. Są tutaj z nami posłowie PiS-u. To jest tak, jakby w ciągu miesiąca zniknęło jedno polskie miasto - Krosno, okręg Marka Kuchcińskiego, czy np. część Kołobrzegu, okręg pana posła Pawła Szefernakera. To jest dzisiaj państwa odpowiedzialność. To nie są zgony, które wynikają wprost z epidemii. To są zgony, które wynikają z tego, że zaniedbaliście przygotowania Polski do czasu epidemii, nie poradziliście sobie z tym i doprowadziliście tych ludzi do śmierci. Taka jest po prostu prawda.

Przecież my słyszymy to zaklinanie rzeczywistości przez pana premiera co jakiś czas. Chociaż pandemia dotyka każdej Polki i każdego Polaka, to są regiony, o których szczególnie zapomnieliście. W październiku 2020 r. zmarło o 83% więcej osób w województwie podkarpackim niż w październiku 2019 r. To są ofiary tego rządu, to są ludzie, którzy nie musieli umrzeć, to są ludzie, którzy umarli dlatego, że system ochrony zdrowia nie był przygotowany. I to są wszystko liczby, które sami przedstawiacie w oficjalnych statystykach. To są liczby podawane przez Główny Urząd Statystyczny, liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Tam wzrost śmiertelności jest często blisko o 100%. To są dane, których nie jesteście w stanie wyjaśnić COVID-em, więc albo nie podajecie precyzyjnych informacji, albo po prostu nie macie informacji na ten temat, a ludzie umierają w domach, umierają w szpitalach i nikt tego w żaden sposób nie jest w stanie wyjaśnić, na pewno nie polski rząd. Województwo podkarpackie, tak jak powiedziałem - wzrost śmiertelności o 83%, województwo małopolskie - wzrost śmiertelności o 67%, województwo świętokrzyskie - wzrost śmiertelności o 63%. To chyba tam najwyższe poparcie miał Zbigniew Ziobro. Śmiertelność wśród osób powyżej 60. roku życia w październiku zwiększyła się o 42%. To, zdaje się, prezydent Andrzej Duda odnosił się bardzo często do ludzi po 60. roku życia. Wy o tych ludziach po porostu zapomnieliście. Dzisiaj ci ludzie pozostawieni są samym sobie. Na 1 tys. mieszkańców wykonujecie 0,88 testów. Na Węgrzech wykonuje się niemal pięć testów na każdy 1 tys. mieszkańców. A więc jeżeli ktoś chciał Budapeszt w Warszawie, to niech bierze przykład z rzeczy, z których warto rzeczywiście brać przykład. I bez względu na to, ile razy powiecie, że wygraliście z wirusem, na koniec roku liczba ofiar koronawirusa w Polsce to będzie [[Dzwonek]] ponad 60 tys. Polaków. I tę najsmutniejszą liczbę od końca II wojny światowej będziemy wam przypominać już do końca, bo to jest wasza odpowiedzialność, wy za to odpowiadacie i wy za to będziecie rozliczeni. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Marek Rutka w imieniu klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Skoro jest tak dobrze, przynajmniej w państwowych mediach, to dlaczego w rzeczywistości jest tak źle? Jednej odpowiedzi na to pytanie oczywiście nie da się udzielić, ale spróbuję wskazać te najważniejsze powody obecnej trudnej sytuacji. Po pierwsze, z epidemią i późniejszą pandemią na taką skalę współczesny świat nie miał do czynienia. Jednocześnie trzeba jasno powiedzieć, że wirus SARS-CoV-2 to nie Ebola, którego śmiertelność przekracza 50%, a w niektórych przypadkach dochodzi do 90%. Rozprzestrzenianie się wirusów można skutecznie ograniczać, ale trzeba do tego szybkiego i mądrego podejmowania decyzji. Niestety w bardzo wielu przypadkach, można powiedzieć, że w zbyt wielu, w naszym kraju nie mieliśmy do czynienia ani z jednym, ani z drugim. Najnowsze doniesienia włoskich lekarzy mówią, że wirus SARS-CoV-2 dotarł do ich kraju już w listopadzie ubiegłego roku. Początkowo lekarze uznali, że czteroletni chłopiec z Mediolanu choruje na odrę, jednak dokładne badania potwierdziły, że dziecko zarażone jest koronawirusem. W styczniu 2020 r. rząd polski dostał notatkę od Agencji Wywiadu, że zagrożenie pochodzącym z Chin koronawirusem jest poważne i należy się przygotować na kryzys. Treść notatki nawet nie była przedmiotem sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W tym czasie komisja zajmowała się różnego rodzaju aferami w służbach. Informacja rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniem epidemicznym w Polsce i Europie na forum Sejmu pojawiła się dopiero 2 marca. Warto wspomnieć, że 25 stycznia, a więc 37 dni przed wspomnianą informacją rządu, wspólnie z grupą posłów Lewicy zgłosiłem interpelację nr 1675 w sprawie ryzyka szerzenia się na terytorium Polski epidemii koronawirusa. To tylko jeden z wielu przykładów, jak spóźnione i nieprofesjonalne były działania władzy. Władzy, która powszechnie uzurpuje sobie monopol na wiedzę i nieomylność. Bardzo często ze strony władzy padały i padają nadal apele w stylu „trzeba się zjednoczyć w walce z epidemią” czy „wszystkie ręce na pokład” Klub Lewicy, jak i ja sam, wspólnie z pozostałymi członkami Komisji Zdrowia wielokrotnie deklarowaliśmy swoją pomoc i chęć, potrzebę rzeczywistej, realnej współpracy nad ograniczeniem rozmiarów i następstw pandemii. Do tej pory nikt z nas, powtarzam: nikt, nie został zaproszony do takiej ponadpartyjnej współpracy w imię zdrowia i życia obywateli i obywatelek. Wezwanie: wszystkie ręce na pokład, w waszym wykonaniu oznacza, że ci, którzy pozytywnie odpowiedzieli na to hasło, zostają automatycznie wyrzuceni za burtę. Mówię to z wielką goryczą. A teraz konkrety. Pacjenci zakażeni COVID-em przywożeni do szpitali wojewódzkich i miejskich, a także powiatowych nie są witani tak, jak w narodowym lazarecie. Wielokrotnie pacjentów na biało-czerwonym stadionie witały kamery rządowej telewizji, a nawet sam pan premier. W tych prawdziwych, realnych szpitalach pacjentów też witają biało-czerwone barwy, ale nie są to kolory stadionu.

Czas oczekiwania wynosił pięć godzin. Czy coś się polepszyło? Niespecjalnie. Przypadek z mojego okręgu sprzed dwóch dni.

Czy ktoś zastanawiał się, czy ktoś zdaje sobie w ogóle z tego sprawę, że aby przetrwać i przeżyć taki transport, trzeba być zdrowym? Jak bogatym państwem musimy być, aby tak marnotrawić gotowość i poświęcenie ludzi i wyłączać karetkę np. na 8 godzin? Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Oferta pracy [[Dzwonek]] na stanowisku ratownika medycznego - 2600 zł brutto. To jest Polska powiatowa, panie ministrze, tak daleka i tak inna od Szpitala Narodowego. To, że system ochrony zdrowia w naszym kraju jeszcze jako tako funkcjonuje, to zasługa ludzi, ich ofiarności, poświęcenia i etosu. To im należy się największy szacunek i uznanie. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dzisiaj wysłuchujemy informacji premiera z ust pana ministra zdrowia na temat najważniejszy, jaki jest: sytuacja systemu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie koronawirusowi. A proszę zobaczyć, jakie wsparcie pan minister ma po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jedna jedyna pani poseł Bartuś. Proszę poinformować kolegów, że dzisiaj jest ważne spotkanie. Wszyscy mieli czas. Ale jak bronimy Polaków - nie ma nikogo. Takie jest podejście Prawa i Sprawiedliwości. Współczuję, bo to wsparcie jest tylko symboliczne, ale widać je także w państwa pracy. Nie ma Pan wsparcia. Podstawową dewizą w medycynie jest: lepiej zapobiegać, niż leczyć. To jest dewiza, która dotyczy nie tylko medycyny, ale również życia, gospodarki, a także funkcjonowania państwa, szczególnie w tak trudnym czasie jak ogólnoświatowa pandemia. Ale żeby przeciwdziałać, trzeba działać, a tego działania z waszej strony nie było. Nie przygotowaliście Polski na drugą falę epidemii, przebalowaliście wakacje i jesteście świadomi tych błędów.

sanitarnego. Pamiętam.

Mało tego, bagatelizowali problem, zachowywali się nonszalancko. Główny inspektor sanitarny, o którym wspominałem, wypowiadał się w taki sposób, że nawet nie przystoi mi dzisiaj z tej mównicy tego powtórzyć.

Świadczy o tym chociażby załamanie się systemu dostaw, dystrybucji gazów medycznych, przede wszystkim tlenu, a także kwestia dostępu do sieci przez różnych konkurencyjnych dostawców. Pan minister przed chwilą o tym mówił, ale my wiemy, że ta sprawa wywołała ogromny kryzys. My o tym wszystkim wiemy. Dlaczego w wakacje nikt w rządzie, w ministerstwie o tym nie pomyślał, nie przewidział, że przy ogromnym wzroście liczby zakażeń tych gazów medycznych może braknąć? Ten brak schematu działań dotknął nie tylko pacjentów, ale i całe życie społeczne i polską gospodarkę. Wasz schemat działania najlepiej opisał pan redaktor Reszka, opisując przykładowo szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

Niech pan minister dzisiaj jasno powie i wyjaśni, kto dostanie te słynne dodatki, te premie. Czy taki dodatek dostanie pani salowa, która od marca ciężko pracuje na oddziale, dba o czystość, ma mnóstwo pracy? Czy taki dodatek dostanie pani pielęgniarka, która nie została skierowana do pracy przez wojewodę, ale pracuje tak samo ciężko jak i ta druga, która została skierowana? A może lekarz, który pracuje w szpitalu powiatowym w szpitalnym oddziale ratunkowym? A może pracownicy techniczni, którzy dostarczają m.in. wspomniane gazy medyczne, wożą butle z tlenem, może oni dostaną? A może dostaną pracownicy DPS-u? A może dostaną osoby, które są opiekunami medycznymi? To osoby, które opiekują się chorym pacjentem od samego przyjęcia do szpitala, a czasem aż do samego końca, do jego śmierci. Opiekun medyczny jest jedyną osobą, która towarzyszy w ostatnich dniach życia osobie chorej, bo rodzina nie może w tym czasie być w szpitalu. Proszę odpowiedzieć, czy te osoby dostaną swoje wsparcie. Między innymi kiedy mówiliśmy, że niepotrzebnie pobiera się podatek od pracowników, którzy mają szczepienia za darmo od swojego pracodawcy - zmieniliście to szybko. Kiedy mówiliśmy, że OSP trzeba dołączyć do tych służb mundurowych, które muszą mieć 100% pensji, kiedy znajdą się w izolacji lub kwarantannie - dołączyliście OSP. A więc proponujemy, [[Dzwonek]] żebyście inne kwestie także zmienili. Pan minister, jeżeli śledzi sytuację i słowa opozycji, wie, o czym mówię. Gdybym miał więcej czasu, chętnie bym wszystkie panu ministrowi przedstawił. Bardzo proszę. W maju tutaj, na ten sali, mówiliście już państwo triumfalnym tonem o epidemii w czasie przeszłym. To był pan premier Morawiecki. Ja wtedy pytałem, na jakiej podstawie. Jeśli już ogłaszamy koniec pandemii, to. Pokazywałem wykresy z innych krajów, gdzie ewidentnie mieliśmy już do czynienia ze spadkiem tej pierwszej fali, można tak powiedzieć.

U nas był ciągle utrzymujący się wysoki stopień, wysoki wskaźnik zakażeń.

Tymczasem w tej chwili Szwecja ma w przeliczeniu na milion mieszkańców niecałe 31 tys. zakażonych, a Polska - nieco ponad 29 tys. Myślę, że do końca roku przegonimy Szwecję albo co najmniej dogonimy w tej statystyce. Szwecja nie zamykała gospodarki, Szwecja nie zadusiła sobie przedsiębiorstw, albo zrobiła to w znacznie mniejszym stopniu niż Polska, więc osiągniemy dokładnie ten sam rezultat, tylko gigantycznym kosztem, o czym wcześniej ostrzegaliśmy. Dlaczego wtedy nie słuchaliście porad specjalistów, którzy mówili, żeby pójść właśnie tą szwedzką drogą, że wytworzenie odporności zbiorowej po prostu zadziała? Jeśli chodzi o liczbę zgonów, nadal jesteśmy za Włochami, co pokazuje, że u nas ta epidemia jest znacznie mniej zakaźna, a mimo to sobie z nią nie radzicie. W statystykach zgonów przegoniliśmy już Austrię, Niemcy, Słowację, Danię, z którymi się wcześniej porównywaliśmy. A my jednocześnie nie dość, że uruchamiamy gigantyczne, często niepotrzebne programy, jak pokazówka na narodowym, i kupujemy rekordowo drogie testy, droższe niż w Niemczech, to jednocześnie dusimy sobie gospodarkę, której nie pozwalamy zarabiać na to, żebyśmy mieli za co z tą pandemią walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Rozumiem, że już zdrowy. Panie Ministrze! Jak już poseł Dobromir Sośnierz powiedział, niestety nie słuchano specjalistów, którzy mówili o tym, że do tego scenariusza i tak dojdzie. W tym momencie oczywiście to się odbywa. Zamknęliście państwo gospodarkę, zamknęliście państwo wybiórczo pewne gałęzie gospodarki.

Jak pytaliśmy o zasadność noszenia maseczek, pokazując informację ze strony WHO, że te maseczki w przestrzeni publicznej są kompletnie bez sensu, to szef GIS-u będący na spotkaniu powiedział: Proszę państwa, no te maseczki mają być przede wszystkim symbolem, żeby lud wiedział, że trwa jakaś pandemia. Jak zasugerowaliśmy, że może warto byłoby chociaż przeczytać Great Barrington Declaration, to jeden z ministrów obecnych na spotkaniu z premierem Morawieckim i z naszymi posłami, powiedział do jednego z naszych posłów, cytuję: Pan jest jeszcze młody, więc może się pan nie przejmuje, ale proszę pomyśleć o swoich dziadkach. Tak infantylna, prymitywna odpowiedź w tak poważnej dyskusji o całym społeczeństwie to było coś, co powinno tego człowieka zwyczajnie wykluczyć z dyskusji w tamtym czasie. Nie macie państwo dobrego rozwiązania. Zniszczyliście państwo gospodarkę.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, poseł niezależna. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Ja tradycyjnie z pytaniem o osoby w kryzysie bezdomności. W jaki sposób one będą szczepione? Na stronie ministerstwa, stronie narodowego programu szczepień czytamy, że do szczepienia będzie kwalifikował lekarz, czyli mamy tę samą sytuację co w przypadku testów. Osoby, najczęściej nieubezpieczone, w kryzysie bezdomności nie są w stanie otrzymać świadczenia, które powinno być powszechne i według deklaracji rzecznika Ministerstwa Zdrowia - bezpłatne, ponieważ muszą przejść przez ten etap kwalifikacji u lekarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę osób zgłoszonych do zadania pytania. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwsza pytanie zada pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewica. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Pandemia stała się ważnym testem dla sprawdzenia stanu przygotowania instytucji państwowych w kryzysie. Rzeczywistość ta pokazała również, jak dramatyczna jest sytuacja podmiotów leczniczych, szpitali, przychodni, poradni i innych jednostek służby zdrowia. Rzecznik praw obywatelskich nieustannie odbiera skargi, że brakuje wolnych miejsc w szpitalach, brakuje sprzętu medycznego, personelu i jednolitych procedur, a personel medyczny stanowi część tego systemu tworzącego solidarność społeczną i bez przywrócenia im należytego, godnego wynagrodzenia ten system nigdy nie ulegnie zmianie. Utrzymujące się od lat niskie płace wymuszają wiele godzin pracy dla pokrycia kosztów kadrowych. Gdyby medycy, pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni pracowali po 8 godzin, system ochrony zdrowia dawno by się załamał i zadławił.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Nie wiem, jak bardzo pan minister chciałby opowiadać, że w służbie zdrowia w Polsce jest dobrze. Tak dobrze nie jest i nie dotyczy to tylko elementów tego systemu, ale od zachodniego Pomorza po Podkarpacie jesteśmy w sytuacji krytycznej, a szczególnie widać to w oddziałach szpitali powiatowych. Tam na oddziałach nie-COVID-owych dzieją się sytuacje niespotykane. Odmawia się przyjęcia pacjentów. Mówi się, że poczekamy, aż będzie szczepionka. Ktoś, kto ma zdiagnozowaną chorobę onkologiczną, słyszy, że musi poczekać parę miesięcy. Inne osoby są odsuwane od szpitali do szpitali. Zwracam się zatem z konkretnym pytaniem w imieniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, jaka pomoc Ministerstwa Zdrowia została skierowana do szpitali powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obecnie cały ciężar walki z epidemią spoczywa na szpitalach publicznej służby zdrowia, na szpitalach, które w większości są poważnie zadłużone lub balansują na krawędzi zapaści finansowej. Chodzi o środki, by walczyć nie tylko z epidemią, ale również, by walczyć o zdrowie i życie pacjentek i pacjentów chorujących na inne, bardzo poważne schorzenia. Dlatego poproszę o odpowiedzi, najlepiej na piśmie: Kiedy rząd zapewni bezpieczeństwo finansowe zadłużonym szpitalom, tak aby mogły skupić się na skutecznym leczeniu pacjentów? Jakie to będą kroki i w jakim terminie podjęte? Jakie konkretne środki są przewidziane dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim? Szczególnie interesują mnie szpitale powiatowe w Ostródzie, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Iława, Bartoszyce, Braniewo, Lidzbark Warmiński oraz Elbląg. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, klub Lewicy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Wystąpiłem w jakimś propagandowym kabarecie i jestem wściekły, bo mnie oszukano. Przyjechałem tu pomagać ludziom, tymczasem mieszkam w 5-gwiazdkowym hotelu, jednym z najdroższych w Warszawie i siedzę w pustym szpitalu. Zarobki są wysokie, koszty funkcjonowania ogromne. To oczywiście głos właśnie tego lekarza ze Szpitala Narodowego, który przyjechał: Jest mi wstyd, że w tym uczestniczę. A więc porównanie. Zarobki ratownika za miesiąc w Bielsku-Białej - 2 tys. zł brutto, zarobki w Szpitalu Narodowym za 84 godziny - 12 600 zł. Dostępność łóżka na Narodowym - 822 zł, dostępność stanowiska z wentylacją - 3700 zł. Proszę o porównanie, ile kosztuje leczenie jednego pacjenta w szpitalu na Stadionie Narodowym i w szpitalu w Koszalinie. Drugie pytanie.

Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Doktryną rządów SLD, Platformy Obywatelskiej i PSL-u przy łataniu dziury budżetowej była prywatyzacja. To właśnie z prywatyzacji polskich firm tę dziurę zasypywano. Mimo sprzeciwu społecznego sam uczestniczyłem w takich akcjach m.in. polski Lotos przeciwko prywatyzacji Lasów Państwowych. Chciałem zapytać: Jakie wpływy, jakie kwoty właśnie spółki Skarbu Państwa przekazały na walkę z koronawirusem i jakie są planowane w tym zakresie? I w tym miejscu również, panie ministrze, w imieniu mieszkańców południowej części województwa łódzkiego, powiatu pajęczańskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego pragnę bardzo serdecznie podziękować, bo dzisiaj dobre wieści dopłynęły do Wielunia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak wiemy, szczepionki nie są jeszcze na tyle nowoczesne, że same się przywożą i organizują szczepienia, dlatego mam kilka pytań. Czy rząd jest już w trakcie przygotowań całego procesu wyszczepienia, od zamówienia konkretnego preparatu po wkłucie igły?

Czy wyznaczone są osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych etapów? Jak obecnie wygląda realizacja tych zadań?

Pan poseł Krzysztof Śmiszek, klub Lewica. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Pandemia koronawirusa obnażyła wszystkie patologie systemu ochrony zdrowia. Przed pandemią nasz system ochrony zdrowia był pod kroplówką, dzisiaj leży pod respiratorem. Dramatyczne niedostatki próbują łatać sami obywatele, organizując zrzutki, zbiórki.

Średnia wieku to 52 lata. Dramatycznie maleje liczba pielęgniarek w szpitalach.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani marszałek. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Żeby wyleczyć pacjenta, potrzebne jest zaufanie pacjenta do lekarza. Żeby pokonać pandemię, potrzebne jest zaufanie obywateli do rządu. A to zaufanie zostało zawiedzione. Na początku pandemii słyszeliśmy, że ona do Polski nie przyjdzie, potem słyszeliśmy, że nie będzie groźna, potem słyszeliśmy, że nie potrzeba testować. Potem zamknięto lasy, co dla Polaków było niezrozumiałe. Potem znowu kazano restrykcyjnie nosić maseczki, ciągle robiliśmy mało testów. Potem w maju okazało się, że pandemia odeszła i mamy czuć się bezpiecznie. Polacy nie wiedzieli w końcu, czy mają uważać, czy nie, stracili zaufanie. Na dodatek kolejki w szpitalach, karetki jeżdżące tam i z powrotem, niemogące zostawić pacjenta w szpitalu, bo nie było miejsca. A nie jest w porządku. Do polityków jest najmniejsze zaufanie w naszym kraju. Dziękuję, pani marszałek. Bardzo proszę. Chcę zderzyć dwa podmioty: Szpital Narodowy i szpital powiatowy. Co miesiąc zarząd tego szpitala kosztuje polskich podatników 629 tys. zł.

Panie Ministrze! Aby utrzymać funkcjonalność szpitala właśnie w Kłodzku, Rada Powiatu Kłodzkiego ostatnio na sesji przekazała 2900 tys. zł.

Finansowanie szpitali jest [[Dzwonek]] obowiązkiem państwa. To konstytucyjny obowiązek, z którego rząd się nie wywiązuje. Chcę zapytać, ile jeszcze, jak długo jeszcze będziecie z jednej strony marnotrawić publiczne pieniądze, a z drugiej strony wykorzystywać samorządy, by te ratowały służbę zdrowia i dostęp do świadczeń zdrowotnych mieszkańców.

Mamy naszą własną Lombardię, mamy nasz własny Wuhan, mamy naszą sytuację, w której nikt nie panował nad tym, że koronawirus w tej drugiej fali, która tak naprawdę jest przedłużoną pierwszą falą, zapanuje nad polskim społeczeństwem. Rzeczywiście naszą nadzieją są szczepienia, dlatego warto zachęcać wszystkich do szczepień. Ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego jesteśmy chyba jedynym krajem z tych, o których czytałam, w którym służby mundurowe są przed pracownikami socjalnymi. Nie umiem zrozumieć, jakie priorytety ma ten rząd. Jeśli chcemy puścić dzieci do szkół, musimy szczepić np. nauczycieli.

Jedyna Pani Posłanko z PiS! Wysoka Izbo! Parę miesięcy temu z tej mównicy mówiłam, że Polki i Polacy boją się pandemii, ale jeszcze bardziej boją się pandemii pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Niestety miałam rację. Przekręty, oszustwa, fake newsy i antyszczepionkowa propaganda siana przez czołowych polityków PiS, łącznie z prezydentem, informacje o lodzie w majtkach, idiotyczne zakazy i brak realnego wsparcia pracowników ochrony zdrowia pokazują, że wprowadziliście chaos większy niż pandemia. Rozumiem, panie ministrze, że pan jest po to, żeby to wszystko po panu Szumowskim posprzątać. Stąd konkretne pytania, panie ministrze. Skoro tak, skoro pan jest od posprzątania, to jakie ma pan plany na wzmocnienie pracowników ochrony zdrowia, by lepiej zarabiali, czuli się bezpieczniejsi, by było ich więcej? Bo dzisiaj wiemy, że te dodatkowe świadczenia dla wybranych nie są zbyt skuteczne, nie pomagają nowym pracownikom. Zapomnieliście o wszystkim innym. Panie ministrze, proszę o odpowiedź na piśmie, ile osób miało odłożone operacje kardiologiczne i onkologiczne, ile osób przez to, że pozamykaliście szpitale w sposób chaotyczny, tej niezbędnej pomocy, często ratującej życie, nie otrzymało. Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, o konkretne informacje. Dziękuję. Pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Bardzo się cieszę, panie ministrze, że pan jest i mogę panu powiedzieć, co się dzieje w województwie świętokrzyskim, bo myślę, że pan po prostu o tym nie wie. Otóż w województwie świętokrzyskim tak się zadziało, że szpital w Skarżysku-Kamiennej stał się szpitalem COVID-owym raptem tylko na 3 tygodnie. Choć ostrzegaliśmy wojewodę świętokrzyskiego, że to jest nieracjonalna i zła decyzja dla mieszkańców, bo wokół jest wiele powiatów, które będą pozbawione dostępu do leczenia w szpitalu wieloprofilowym, pan wojewoda nie słuchał. Po 3 tygodniach przyznał nam rację. To nie wszystko.

Może kiedyś wrócą, a może nie. Otóż, panie ministrze, [[Dzwonek]] w Starachowicach były kliniki serca. Zostały zlikwidowane.

Bardzo proszę.

Wysoki Sejmie! Prosił pan w swoim wystąpieniu, abyśmy rozmawiali tylko o faktach. Fakt pierwszy, 2 listopada. Na trasie z Włodawy do Chełma dochodzi do wypadku.

Następnie zabierani są karetką do szpitala w Chełmie. Nie mogą być przyjęci z powodu braku miejsc. Jakie są konsekwencje? Obaj umierają w karetce. Fakt drugi, początek listopada. Fakt trzeci, połowa listopada. Kolejka przed jednym ze szpitali w Lublinie na 20 godzin. Ratownicy medyczni mówią o tym, że wolą udzielać pomocy osobom chorym na COVID w domu (Dzwonek), niż zabierać ich do kartki, bo będą musieli kilkanaście lub 20 godzin czekać w tej karetce.

Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pierwszy fakt jest taki, że od 26 sierpnia nie widziano posła Łukasza Szumowskiego. Tak kończą, szanowni państwo, ministrowie, którzy podają się do dymisji bez wyjaśnienia spraw.

Bo to jest manko, które pan ma w budżecie resortu zdrowia, to są środki, które miały być zwrócone w respiratorach, a nie zostały zwrócone. Czy umowa na respiratory była opiniowana przez Prokuratorię Generalną? Jakie były podejmowane działania od czasu podpisania umowy, [[Dzwonek]] tak naprawdę od końca czerwca, na rzecz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa? Dziękuję. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie Ministrze!

Chciałbym zadać pytanie w związku z informacjami o szczepionkach. Mówi pan, że będą ułatwienia dla tych, którzy się zaszczepią. A co z tymi, którzy przeszli chorobę i mają naturalną odporność w wyniku infekcji, uzyskali przeciwciała?

Po pierwsze, to było nierównomierne, że tak powiem, wykorzystanie tej bazy. I oczywiście szpitale w chwili obecnej mają ten problem, że część kadry zaczyna uciekać i chciałaby wrócić do niektórych funkcji.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie Ministrze! Kilka wniosków. Po pierwsze, ferie powinny być organizowane przez 8 tygodni, nie przez 2 - tu będziemy polemizować - ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Druga sprawa to szczepienia.

Może nawet niedowiarka Andrzeja Dudę uda się przekonać do tego, żeby się zaszczepił. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to otwarcie prywatnej służby zdrowia.

Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pierwsza sprawa. Wczoraj na liście wniosków rządowego programu inwestycji lokalnych został pominięty wniosek z Rawy Mazowieckiej dotyczący szpitala. Panie ministrze, bardzo pana proszę o interwencję w tej sprawie.

Na razie te, które pan przedstawił wczoraj na komisji i w dokumencie dotyczącym strategii, są naprawdę bardzo ubogie. Pytanie, czy pan zamierza rozszerzyć ten wachlarz.

Panie ministrze, czy to jest możliwe?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zacznę od tego, co tutaj przed momentem wybrzmiało, ale było też przywoływane wcześniej, że jestem jedynym posłem PiS, który jest na sali. Czy pani marszałek nie jest z PiS-u? Czy pan poseł, który siedzi tutaj.

Szanowni Państwo!

Z jednej strony wychodzicie i mówicie: było za mało zachorowań, za dużo zachorowań. Szanowni Państwo! Mamy brać udział w debacie, czy nie? Mam pytanie.

Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo!

Każdemu z parlamentarzystów wydłużałam czas, nikomu nie wyłączałam mikrofonu. Proszę o tym pamiętać i być sprawiedliwym. Pani poseł, ja już skończyłam w tej sprawie. Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Chciałam zapytać o branżę turystyczną, która jest w całkowitej zapaści. Przedsiębiorcy są przygotowani do sezonu zimowego. Tymczasem branża została całkowicie zamknięta. Moje pytanie, panie ministrze: Jakie są szanse przy zabezpieczeniu i zagwarantowaniu tego, jeżeli chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo turystów, a także mieszkańców, że zgodzi się pan, żeby zmniejszyć trochę te restrykcje, znieść ograniczenia, bo w przeciwnym razie to będzie całkowite, wielkie bankructwo? Powiem tylko, że Czesi otworzyli całkowicie sezon. Owszem, są ograniczenia. I ja nie apeluję, żeby znieść wszystkie ograniczenia. Czy my chcemy, żeby wszyscy turyści pojechali do Czech (Dzwonek), czy chcemy pozbawić przychodów naszych przedsiębiorców i pozbawić turystów możliwości wypoczynku? Przecież wielu z nich już jest po zachorowaniach. Bardzo proszę, aby pan dzisiaj na to odpowiedział, bo przedsiębiorcy i mieszkańcy czekają na to, jaką odpowiedź ja im przekażę.

Pragnę przypomnieć, proszę to sprawdzić, ile czasu otrzymała pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz, która zadawała bardzo merytoryczne pytanie, dlatego w żaden sposób zakres ten nie był ograniczany.

Jest świetnie przygotowana, są ludzie, jest zaplecze, są możliwe różne usługi, jest nawet część zaplecza takiego medycznego, a przede wszystkim wsparlibyśmy biznes.

Ale czy prowadzi pan dodatkowe szkolenia, przygotowania kadr? Ja wiem, że nie wykształci się w pełni służb przygotowanych do usług medycznych, ale do pomocy jest to możliwe. Szereg osób, jeśliby miałoby szansę na pracę, podjęłoby takie kursy. To dzięki nim funkcjonują budowy i różne branże, tworzy się PKB. Na ile pan zabezpieczy wsparcie dla tej grupy osób, bo oni są dobrem dla polskiej gospodarki? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Moje pytanie jest bardzo proste: Jaki jest sens budować te szpitale tymczasowe, które de facto, jeśli ulokowane są w pomieszczeniach nieprzystosowanych do funkcji szpitalnych, medycznych, służą wyłącznie jako bardzo drogie i bardzo kosztowne izolatoria? Koszt szacowany jest na ok. 40 mln.

Czy nie lepiej byłoby zagospodarować, odświeżyć te budynki, które mają pełne oprzyrządowanie, pełną infrastrukturę do pełnienia funkcji pełnowartościowych szpitali COVID-owych, a nie budować kolejne kosztowne izolatorium w partnerstwie z prywatnym [[Dzwonek]] przedsiębiorcą? Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, ja jestem pracownikiem wojewódzkiego szpitala obserwacyjno-zakaźnego, szpitala, w którym funkcjonują dwie kliniki zakaźne. Zatem mam bezpośredni kontakt z ludźmi frontowymi, którzy na co dzień są z koronawirusem. Wie pan, o co oni mnie prosili?

Oni dostają mniej więcej minimalne wynagrodzenie w naszym kraju. Czy pan minister myśli o tych, którzy tworzą organizm tego szpitala? Bez ich pracy nie byłby możliwy (Dzwonek) wysiłek lekarzy i pielęgniarek przy ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Apeluję do pana ministra, aby pan minister pochylił się bardzo mocno nad tym, co powiedziałem. Dziękuję bardzo. Pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Bardzo proszę, panie pośle.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiemy, że sytuacja z koronawirusem w kraju nie jest prosta, ale chciałbym zapytać pana ministra, czemu mają służyć te spektakularne akcje, które prowadzicie od wiosny. Najpierw witanie płynu, łącznie z oceną organoleptyczną płynu na Orlenie, później maseczki transportowane antonowem, teraz urządzanie szpitali tymczasowych na stadionach, gdy stoją puste szpitale: szpital południowy w Warszawie, szpital w Katowicach, szpital w Łodzi, szpitale w Białymstoku, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szkoła.

Teraz już do tej nauki zdalnej trochę się przyzwyczailiśmy, chociaż oczywiście nam się to nie podoba, nikomu się to nie podoba.

Nie chciałbym usłyszeć, że planujemy, zastanawiamy się, zobaczymy, sprawdzimy. Chciałbym, żeby pan powiedział, że jest scenariusz wychodzenia z tego kryzysu dla polskiej edukacji. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie w tym punkcie zada pan poseł Marek Rutka, klub Lewica. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Decyzją wojewody pomorskiego szpital powiatowy w Pucku został przekształcony w tzw. szpital COVID-owy. Biorąc udział w jednym z programów telewizyjnych, odpowiedziałem na apel pani Olgi Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, aby włączyć się w prace nad zwalczaniem skutków epidemii. Kilkukrotnie zwróciłem się do pani minister z prośbą o dostarczenie środków czystości, papieru toaletowego, podkładów medycznych do szpitala powiatowego w Pucku. Żadnego odzewu, żadnego kontaktu. W związku z tym ze współpracownikami zakupiliśmy środki czystości dla tego szpitala, ale wystarczyło to zaledwie na 2 dni.

Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O udzielenie odpowiedzi na postawione pytania bardzo proszę ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego.

Bardzo proszę. Szanowni Państwo! Z wielką uwagą i atencją wysłuchałem wszystkich tych uwag. Cały czas chcę deklarować, że moja otwartość na współpracę jest otwartością na każdą rozmowę, na każdą dyskusję, również na spotkania, na wymianę argumentów - bo niestety wszyscy widzimy, że dyskusja na temat COVID-u jest polityczna od samego początku. Oczywiście staram się tę politykę oddzielić, bo COVID nie ma barwy politycznej, COVID dotyka każdego. No może częściej i z większymi skutkami dotyka osoby, które dotyka wielochorobowość bądź które są w zaawansowanym wieku. Ale chociażby przekrój państwa pytań i komentarzy, opinii pokazuje, jakim wyzwaniem, jak kompleksowym zagadnieniem jest walka z pandemią. To dotyczy bardzo różnych wymiarów funkcjonowania państwa, bo to są po prostu naczynia połączone.

To są oczywiście zgony. Zgony są największą troską nie tylko ministra zdrowia, ale też oczywiście medyków, całego personelu. To jest zagadnienie, które w tej chwili jest najważniejsze, to jest priorytet priorytetów. Nie interpretujmy tych zgonów w sposób polityczny, nie interpretujmy ich w ten sposób, żeby obciążać je polityczną barwą, bo to są tragedie ludzi, to są tragedie rodzin, to są tragedie, które w zasadzie, patrząc na liczbę zgonów, dotknęły bardzo, bardzo wiele rodzin w Polsce. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów, rzeczywiście pandemia przyczyniła się nie tylko w sposób bezpośredni, ale również w sposób pośredni do zwiększenia liczby zgonów w Polsce.

Analizowaliśmy bardzo dokładnie ten problem, bo, jak powiedziałem, ma on dla nas charakter priorytetowy. Wychodzi na to, że co najmniej jeszcze 10%, kolejne 20% tych zgonów jest związanych pośrednio z COVID-em, tzn. pośrednio w ten sposób, że u ludzi, którzy chorują na COVID, w przypadku wielochorobowości i w przypadku wieku zaawansowanego niestety odnotowujemy zgony mniej więcej po 30 i więcej dniach po przechorowaniu COVID-u.

Musimy też powiedzieć sobie otwarcie, że część tych zgonów jest związana z ograniczeniem dostępu do ochrony zdrowia, bo musieliśmy przeznaczyć część zasobów, część łóżek szpitalnych na to, żeby hospitalizować tych pacjentów, którzy są właśnie w najcięższych stanach COVID-owych. Tutaj nie ma możliwości powiększania w nieskończoność bazy łóżkowej, tutaj trzeba zarządzać ograniczonymi zasobami.

Chcę zwrócić państwa uwagę na to, że paradoksalnie szpitale tymczasowe są bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej, ponieważ one mogą przejmować część opieki nad lżej chorymi, nad tymi, którzy wychodzą ze stanu ciężkiego, nie obciążając standardowej infrastruktury szpitalnej, którą możemy przeznaczyć czy dedykować po prostu leczeniu standardowych chorób, z którymi również musimy sobie radzić. Nadal głównym zabójcą w Polsce są choroby kardiologiczne, nadal onkologia jest dominującym, drugim, jeśli chodzi o liczbę zgonów, zabójcą w Polsce. Dlatego tak szybko trzeba redukować tę liczbę łóżek i dlatego zdarzają się sytuacje, w których na 3 tygodnie jakiś szpital został COVID-owym. Z mojego punktu widzenia to jest odzwierciedlenie dobrego zarządzania infrastrukturą szpitalną, ponieważ jak tylko można było, te łóżka zostały przeznaczone na leczenie tych głównych zabójców w Polsce. Ponieważ zgony są najważniejszym wyzwaniem, na którym się koncentrujemy, to oczywiście oprócz analizy podjęliśmy badania i działania. Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że od mniej więcej 2 tygodni zostały zmienione wytyczne dla zespołów ratownictwa medycznego dotyczące zabierania pacjentów z saturacją poniżej 94%. Do tej pory ta liczba odmów - bo też to zagadnienie analizowaliśmy - była niepokojąco duża. Od początku procesu patrzyliśmy, że to są liczby, które osiągały wolumeny rzędu tysięcy, więc wprowadziliśmy nowe wytyczne, które nakazują jednoznacznie zabierać pacjenta z saturacją poniżej 94%, i mamy pierwsze tego efekty. Chętnie w odpowiedziach pisemnych przedstawię państwu też wykresy, które pokazują, jak po wydaniu tych wytycznych rozchodzi się właśnie krzywa liczby odmów i krzywa transportów czy pacjentów transportowanych do szpitala. Bo według specjalistów, według Rady Medycznej przy panu premierze główną przyczyną rosnącej liczby zgonów w zakresie COVID-owym jest zbyt późny transport pacjenta do szpitala. Żeby to zrobić, zainteresowaliśmy się działaniem zespołów ratownictwa medycznego, analizując dokładnie, jak wyglądają poszczególne kroki, czasy oczekiwania, co jest problemem przy transporcie pacjentów. Dlatego oprócz tych wytycznych powstał specjalny system informatyczny, który na zasadzie rezerwowania miejsc pokazywał zajętość łóżek w poszczególnych szpitalach. To było nowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy 2 miesiące temu czy 1,5 miesiąca temu, ale ponieważ jakość informacji wprowadzonych do tych systemów budziła wątpliwości, zdecydowałem w porozumieniu z ministrem obrony o wysłaniu żołnierzy wojsk ochrony terytorialnej, żeby obiektywną informacją zasilali ten system, ale oczywiście też odciążyli pracowników szpitali od administracyjnej, biurokratycznej pracy. Druga odpowiedź dotycząca tego, żeby pacjent trafiał w odpowiednim momencie do szpitala, to jest masowy program, który uruchomiliśmy. Myślę, że będzie to jeden z powodów do zadowolenia dla nas, jako dla państwa, bo będzie to masowy program, niespotykany w skali europejskiej - to jest domowa opieka medyczna przy wykorzystaniu pulsoksymetrów, czyli urządzeń, które służą do monitorowania saturacji, czyli natlenienia krwi. To te urządzenia, które przy pomocy smartfona i specjalnej aplikacji przesyłają dane do centrum monitoringu, mają poinformować siedzących tam lekarzy i konsultantów, że dzieje się coś niedobrego, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Patrząc na statystyki tego programu, chcę państwu powiedzieć, że w ciągu kilku tygodni jego funkcjonowania udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że w tej chwili mamy objętych programem blisko 30 tys. pacjentów. Jest blisko 30 tys. pacjentów, do każdego z nich został wysłany pulsoksymetr, każdy z nich będzie aktywowany i informacja będzie przesyłana do centrum monitoringu. Niestety mieliśmy też sytuację, że w ponad 30 przypadkach - ale temu miał służyć ten program - były wysyłane załogi ratownictwa medycznego właśnie do pacjentów objętych tym programem.

Szpital tymczasowy i jego wycena, która została zresztą sporządzona przez wyspecjalizowaną instytucję, którą do tego mamy, czyli Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jest szpitalem, który jest finansowany tylko i wyłącznie ze stawek dziennych, które właśnie w wycenie tej instytucji się znalazły. Nie można porównywać tego z wyceną chorego, który jest, że tak powiem, opłacany w szpitalu np. powiatowym, tak jak państwo podawaliście, bo szpital powiatowy oprócz stawki za pacjenta otrzymuje całą długą listę przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia, zaczynając najczęściej od ryczałtu, czyli stałej płatności, powiększając to o opłatę z tytułu gotowości, o rekompensaty różnego rodzaju, gdzie opłata fee for service dochodzi jako krańcowa wartość w tym, co otrzymuje sumarycznie szpital ze strony NFZ. Szpital tymczasowy nie ma przychodów, ma tylko i wyłącznie stawkę za pacjenta, więc ta stawka musi rekompensować wszystkie kategorie kosztów, które szpital powiatowy ma zrekompensowane w formie ryczałtu, który pokrywa przecież wszystkie wynagrodzenia, czy w formie innych opłat za gotowość, które są płacone w sieci COVID-owej. Tak że jeżelibyśmy sobie te koszty porównali i dołączyli w szpitalu powiatowym do stawki wszystkie te komponenty kosztowe, to mielibyśmy porównywalną wycenę, porównywalną cenę.

Postaram się to wyjaśnić w sposób możliwie prosty. Otóż mamy dwie grupy personelu medycznego, któremu płacimy dodatki. Jeden to jest personel, który jest kierowany przez wojewodę, i wtedy mamy regulację ustawową, która jest podstawą wypłacania tego dodatku, i każda osoba skierowana przez wojewodę do pracy w związku z COVID otrzymuje taki dodatek - każda. Czy to będzie lekarz, czy to będzie pielęgniarka, czy to będzie ratownik medyczny, każde z nich otrzyma taki dodatek.

Tutaj mamy upoważnioną grupę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, którzy pracują w laboratoriach szpitalnych. W stosunku do poprzedniego rozwiązania powiększyliśmy tę grupę właśnie o ratowników i o diagnostów laboratoryjnych. Ale, co ważne, wcześniej te pieniądze były wypłacane tylko i wyłącznie osobom, które wyłącznie, podkreślam, walczyły z COVID-em. Teraz nie muszą wyłącznie tu pracować - jeżeli idą na inny oddział, to nie tracą tego dodatku, będą go otrzymywały. Ponieważ wiedziałem, że dzisiaj padną pytania na ten temat, przygotowując się do spotkania z państwem, poprosiłem Narodowy Fundusz Zdrowia o podsumowanie, jak wygląda kwestia wypłacania tego dodatku na podstawie realizowanego polecenia.

Suma kwot zgłoszonego zapotrzebowania na środki.

Zapotrzebowanie już zgłoszone w ramach wypłacenia tych wydatków to jest 40 mln zł za miesiąc na dodatki dla personelu. Szanowni Państwo! Przechodząc do następnego zagadnienia, chciałbym, żeby nasze rozmowy na temat pandemii, na temat walki z COVID-em toczyły się w oparciu o fakt, w oparciu o liczby, w oparciu o wzajemny szacunek, o nie przekrzykiwanie się, tylko rzetelną dyskusję. Dlaczego? Dlatego, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wygenerować pewien kapitał polityczny, o którym mówiła pani poseł Kidawa-Błońska. Kapitał społeczny, który będzie budował zaufanie, które jest szczególnie ważne w kontekście szczepień, które nas czekają. Naprawdę nie zachowujmy się jak małe dzieci, które odmrożą sobie na złość rodzicom uszy, i nie grajmy pewnymi wartościami, które potem odbijają się na zdrowiu publicznym w Polsce. Mówimy tu o zdrowiu, nie o światopoglądzie - o zdrowiu.

Szanowni państwo, bardzo proszę, jeśli państwa to nie interesuje, to można zawsze wyjść w kuluary. Rozumiem, że temat został zgłoszony.

Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi o szczepienia, mamy zakontraktowane 62 mln dawek, podkreślam, dawek szczepień. Ponieważ większość tych szczepień wymaga podwójnego dawkowania, więc to w całości zabezpiecza potrzeby populacyjne Polski. To oznacza, że każdy obywatel naszego kraju ma zagwarantowane prawo do zaszczepienia i do niego należy decyzja, bo postanowiliśmy, że decyzja o szczepieniu będzie dobrowolna. Żeby tę decyzję i tę dobrowolność promować, jako państwo bierzemy na siebie większe zobowiązanie, bo musimy obywateli przekonać. Przekonać, po pierwsze, że szczepienie jest bezpieczne, a po drugie, że korzyści z zaszczepienia to są korzyści, które nie dotyczą tylko zdrowia, nie dotyczą tylko odporności populacji, ale chodzi o to - co przewijało się jako wątek w państwa wypowiedziach - by również powrócić do normalnego funkcjonowania gospodarki.

Tutaj chodzi o rozwiązania systemowe, o serwisy, o akcje, o kampanie, o namawianie nie w oparciu jedynie o to, że chcemy, żeby ludzie się zaszczepili, tylko o przekazywanie rzetelnej wiedzy, jakie są szczepienia. Zresztą w strategii, którą opublikowaliśmy, która nazywa się: narodowy program szczepień, już naprawdę można znaleźć dużo konkretnej wiedzy na temat szczepień, jakie zakontraktowaliśmy, jakie to są rodzaje, jakie technologie tych szczepień są wykorzystywane.

Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa szczepień, to oczywiście żadne szczepienie, które nie przejdzie certyfikacji, nie przejdzie dopuszczenia do rynku europejskiego, nie będzie przez nas promowane. Jak państwo wiecie, są różne szczepionki funkcjonujące na świecie, dużo się mówi o szczepionce rosyjskiej, chińskiej, ale to są szczepionki niezweryfikowane, które nie przeszły badań klinicznych, i one absolutnie nie mogą być dopuszczone w Polsce do obrotu, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych obywateli. Dopiero po certyfikacji, po dopuszczeniu do obrotu, po decyzji Komisji Europejskiej - bo ona ma tak naprawdę tutaj charakter głosu dopuszczającego - jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni tak naprawdę rozpocząć akcję szczepieniową. Kolejne zagadnienie, które tutaj się przewijało, to są testy i badania.

Szanowni państwo, zdecydowaliśmy się na taki system testowania naszych obywateli, który jest ukierunkowany na testowanie osób objawowych. Dlatego jeśli pandemia wyhamowuje, jeśli mamy mniej osób z objawami, jeżeli mamy mniej zachorowań, to również wykonujemy mniej testów. Ale jak zauważyliśmy, że ta liczba testów z poziomu 80 tys. zaczyna spadać poniżej 50 tys., to żeby jednak utrzymać ten rzetelny poziom testowania w populacji, wprowadziliśmy testy antygenowe. Chciałbym państwu powiedzieć, że w ostatnim czasie kupiliśmy blisko 2 mln testów, większość z nich już została rozkolportowana po kraju. Te testy wprowadziliśmy, po pierwsze, w tych miejscach, gdzie trzeba szybko decydować o tym, jaką ścieżką trzeba poprowadzić pacjenta, a więc te testy zostały przekazane do izb przyjęć, do SOR-ów, w kolejnym kroku przekazaliśmy je do karetek, a teraz właśnie trwa rozsyłka dużej liczby testów do DPS-ów, żeby testować zarówno personel, jak i osoby tam się znajdujące. Dzięki temu teraz mamy 40 tys. testów, a nie 20 tys., bo już blisko połowa z tych testów ma charakter testów antygenowych i już nie upieramy się tylko i wyłącznie przy testach PCR-owych. Dlaczego? Dlatego że nie jesteśmy w szczycie pandemii. W szczycie pandemii trzeba było się koncentrować na pacjentach objawowych, a teraz możemy testować więcej i dlatego spada nam wskaźnik trafialności w ramach tych testów. Szanowni państwo - Szwecja. Szwecja jest moim ulubionym tematem, ponieważ robimy do niej różne nawiązania, a obawiam się, że te nawiązania nie bazują na rzetelnej wiedzy. Polecam dzisiejszy artykuł w „Gazecie Wyborczej” - żeby nie było wątpliwości - który mówi o tym, co się dzieje w regionie sztokholmskim.

My tej sytuacji uniknęliśmy. Mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Ten bufor bezpieczeństwa, o którym mówiłem na wstępie. Oczywiście, że pojawiały się sytuacje, o których państwo mówicie. Nie będę malował trawy na zielono.

Naprawdę trzeba docenić pracę wojewodów wykonaną w ciągu pandemii, bo to oni w dużym stopniu decydowali, że te łóżka były dostępne, nawet jeśli system nie działał doskonale. Pani marszałek, już może nie przedłużając wystąpienia.

Nie można powiedzieć, że z pandemią poradziła sobie polityka. Z pandemią poradziliśmy sobie razem. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Pani poseł. Panie ministrze, bardzo dziękuję za długie, ale niezwykle spokojne, a przede wszystkim merytoryczne i rzetelne wystąpienie. Przepraszam za wydłużenie czasu, ale myślę, że Polacy czekali na tę informację, dlatego zdecydowałam się tutaj nie ograniczać w żaden sposób czasowy wystąpienia pana ministra. Zamykam, szanowni państwo, dyskusję. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy na następnym posiedzeniu Sejmu. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Jeśli nikt się nie zgłasza, listę posłów zgłoszonych do oświadczenia uważam za zamkniętą. Jako pierwsza oświadczenie wygłosi pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewica. Zapraszam, pani poseł, do wygłoszenia oświadczenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pandemia koronawirusa zmusiła nas i wiele innych krajów do zamrożenia części gospodarki i życia społecznego. Ale ten okres kiedyś minie i nastąpi odwilż. Jaki obraz ujrzymy, kiedy odpuszczą mrozy obostrzeń i zakazów? Chcielibyśmy wszyscy znów cieszyć się tętniącymi życiem polskimi miastami, miasteczkami i wsiami. Chcielibyśmy znów spotykać się w szkole, w pracy, w restauracji, w kinie. Chcielibyśmy na nowo tchnąć energię w nasze gminy, regiony i aglomeracje, powrócić do spraw, które nam przerwano. Obawiam się jednak, że zastanie nas zupełnie inny widok. Widok uboższy o dużą część publicznej komunikacji zbiorowej, która dzisiaj obumiera w ciszy. Połączenia lokalne są likwidowane i zawieszane z powodu pandemicznych obostrzeń, które nałożono na transport publiczny mimo braku potwierdzenia wysokiego ryzyka przenoszenia wirusa tą drogą. Są one także wstrzymane z powodu zmniejszenia ruchu podyktowanego ogólnymi wskazaniami ograniczenia przemieszczania się, jednakże rząd nie zadbał o to, aby zamrożony transport miał szansę ponownie się podnieść. Zawieszono kursy PKS do Świeradowa-Zdroju, Zielonej Góry czy do Lwówka Śląskiego, w którym wcześniej zlikwidowano już kolej, ale także w Kłodzku, Sieradzu - tu przykład rozkładu jazdy, gdzie żaden z autobusów już nie odjeżdża z tego stanowiska. Wstrzymano rozkłady i linie w Gorzowie Wielkopolskim czy Przemyślu.

Lista problemów sektora transportowego jest długa i część tej listy udało się skierować w formie interpelacji do kilku ministerstw, po spotkaniu z przewoźnikami podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, które to spotkanie odbyło się w połowie listopada. Nasza gospodarka potrzebuje wytyczenia drogi ku nowoczesności, a droga ta prowadzi przez sprawny, bezpieczny, ekologiczny transport publiczny, którego gęsta sieć regularnych połączeń stanie się fundamentem nowej gospodarki. Ku przyszłości musi nas zabrać nowoczesny, szybki i ekologiczny pociąg, podmiejska kolejka, tramwaj czy autobus korzystający z zielonej energii.

Jeśli nie zadbamy o sektor komunikacji publicznej, to wykluczenie transportowe upowszechni się zamiast kurczyć (Dzwonek), a po uchyleniu obostrzeń wiele regionów nie wybudzi się z przymusowego zimowania, bo nic już nie będzie tam dojeżdżać: ani pociąg, ani PKS, a opuszczeni przez własny rząd ludzie będą musieli powrócić do normalności na piechotę. Dziękuję. Dziękuję pani, pani poseł. Muszę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, ponieważ walczycie państwo o prawa kobiet, a kiedy pani poseł wygłaszała ważne oświadczenie, poruszyła ważne tematy, to tu słyszałam śmiechy, chichy, chodzenie, gaworzenie. To nie jest szacunek do kobiet, szanowni państwo. Kolejne oświadczenie, pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z wielkim bólem przyjąłem informację o śmierci Katarzyny Łaniewskiej. Była wybitną aktorką filmową i teatralną oraz działaczką antykomunistyczną i patriotką. Zagrała w ponad 80 filmach i serialach, m.in.: „Godzina W”, „Plebania”, „Czterdziestolatek”, „Klan”, „Smoleńsk”, program „Ziarno” i oczywiście „Kogel-mogel” Słynna scena, w której Katarzyna Łaniewska rozpacza nad zamążpójściem córki, lamentując: oj, córciu, córciu, już ty długo panienką nie będziesz, wpisała się do kodu kulturowego współczesnego pokolenia. Scena ta jest do dzisiaj przytaczana w wielu kontekstach. Jest to niezwykle interesujące, bo pierwszą część „Kogla-mogla” nakręcono 32 lata temu, a pomimo to film ten bawi kolejne rzesze widzów. Mało kto wie, że Katarzyna Łaniewska zajmowała się również dubbingiem. Jej głos możemy usłyszeć w „Wielkiej miłości Balzaca”, „Jeszcze bardziej zgryźliwych tetrykach”, ale również w „Smerfach” czy „101 dalmatyńczykach” Krzepiła ducha, recytując w trakcie mszy św. wiersze. Była mocno zaangażowana w walkę z komunistyczną władzą. To ona założyła „Solidarność” w Teatrze Ateneum. Za tę walkę zresztą została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Katarzyna Łaniewska regularnie upamiętniała ofiary katastrofy smoleńskiej, sympatią darzyła „Gazetę Polską” oraz publikowała felietony w tygodniku „W sieci” Talent artystyczny jest jednak czymś ponad politycznym światopoglądem, dlatego sądzę, że jej śmierć uderzyła tak samo wszystkich Polaków. Dziękujemy za wspaniałe role. Dziękujemy za patriotyzm. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

Panie Ministrze! Chciałbym uprzejmie zasygnalizować panu, że pański poprzednik, pan Łukasz Szumowski, opuszczając w pośpiechu gabinet, zapomniał przekazać panu kluczyk do biurka, w którym są interpelacje, na które pan minister nie udzielił odpowiedzi. I proszę, by zechciał pan się skontaktować z panem ministrem, otworzyć to biurko, bynajmniej nie z ciekawości. Chodzi o to, by otworzyć to biurko, bo to, co pan tam znajdzie, może pana zainteresować w aspekcie dalszego kierowania Ministerstwem Zdrowia, a jest to określone - czasami - regułami polskiego prawa. Otóż tak: 12 czerwca wraz z grupą posłanek i posłów Lewicy skierowałem do pana ministra interpelację w sprawie personalnego wskazania osób odpowiedzialnych w Ministerstwie Zdrowia za zawarcie umowy na zakup 1200 respiratorów za kwotę 200 mln zł od firmy zajmującej się usługami lotniczymi, szkoleniem pilotów, znanej także z handlu bronią, czyli firmy z Lublina. W tej interpelacji pytaliśmy, kto w Ministerstwie Zdrowia zweryfikował wiarygodność i faktyczną zdolność do realizacji tego zamówienia? Kto i na jakiej podstawie zdecydował, że zapłata ma nastąpić z góry? Kto podpisał zlecenie przelewu na 200 mln zł? Kto sprawdził ceny rynkowe respiratorów? I prosiliśmy o wskazanie imienne osób w resorcie, które się pod tym podpisały. Otóż 7 lipca, czyli ponad pół roku temu, pan wiceminister Kraska poinformował panią marszałek, że odpowiedź na te pytania jest niezmiernie skomplikowana, i poprosił o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi, bowiem pan minister był wtedy na etapie pozyskiwania informacji od komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia. Zakładam, że pan wiceminister pozyskał już te informacje. Czy ta informacja jest wstydliwa, czy kogoś obciążająca, że przygotowana odpowiedź na tę interpelację zamiast do grupy posłów trafiła, znalazła się w głębi biurka ówczesnego ministra? Szanowny Panie Ministrze! Jak pokazują na konkretnych przykładach polskie media, wielu handlarzy bronią, narciarzy, wiele żon narciarzy, wielu sprzedawców oscypków czy chińskich producentów podróbek zrobiło na pandemii interes życia dzięki dawanym im lekką ręką (Dzwonek) pieniądzom z Ministerstwa Zdrowia. Zakładam, że panu ministrowi zależy na wyjaśnieniu wszelkich nieprawidłowości i nie ma Pan żadnego interesu w braniu na siebie grzechów poprzednika.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgoła inne oświadczenie, ale dotyczące daty 13 grudnia.

Ale też 13 grudnia 1966 r. w Waszyngtonie zmarł Stanisław Mikołajczyk, działacz ludowy, związkowy, premier rządu na uchodźstwie po tragicznej śmierci gen. Sikorskiego. Był wszędzie tam jako człowiek, jako Polak, obywatel, Wielkopolanin, gdzie wzywała go ojczyzna. Od 1920 r. włącza się w działalność ruchu ludowego - najpierw PSL „Piast”, potem w jego zmianach historycznych, również na uchodźstwie, w okresie wojny oraz okresie powojennym.

Był również prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych.

Tam też jest włączony w skład pierwszej Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej jako wiceprzewodniczący, potem wchodzi w skład rządu, jest wicepremierem, a tak jak powiedziałem, po śmierci gen. Sikorskiego - premierem rządu na uchodźstwie. Walczy z wielką determinacją o powojenny kształt granic powojennej Polski, ale czuje się oszukany przez aliantów, kiedy w 1944 r. w Moskwie dowiaduje się o porozumieniu aliantów z Teheranu i o granicy na linii Curzona. Po konferencji jałtańskiej przystępuje do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej jako wicepremier i minister rolnictwa. Niektórzy traktują to jako zdradę ideałów rządu londyńskiego, a on mówi, że te tysiące czy setki tysięcy młodych Polaków, którzy znajdują się w lasach i z nich nie wyszli, należy ratować dla przyszłości Polski.

Mamy aresztowania, mamy odbieranie gospodarstw, mamy usuwanie z pracy w administracji, ale też codziennością są polityczne mordy. W swej książce „Polska zgwałcona” napisał, że bezpośrednim powodem było przygotowane pozbawienie immunitetu oraz aresztowanie i osądzenie przez sąd wojskowy. Aktywny polityk na emigracji, który napisał w tejże książce „Polska zgwałcona” wielkie przesłanie dla przyszłości: A Polska będzie wolna i demokratyczna. I to jest wielki depozyt tego wielkiego Polaka, Wielkopolanina i również działacza ruchu ludowego dla nas wszystkich. Proszę o wygłoszenie oświadczenia. Przewodniczący Komitetu Kaczyński! Wysoka Izbo! Panie Premierze Morawiecki! Dziś chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest stan negocjacji z Unią i do czego tak naprawdę dąży nasz rząd. Nie wystarczy wrzucić zdjęcie z tajnej narady z maską na oczach prezesa i uważać, że sprawa jest załatwiona. Nie jest. Moi wyborcy chcą znać prawdę. Niech premier Morawiecki poprowadzi nas przez ten labirynt decyzji podjętych i niepodjętych, jawnych i niejawnych, bo wszyscy się już pogubili. Co zostało ustalone na prywatnym szczycie między prezesem PiS-u Kaczyńskim a przewodniczącym Fideszu Orbánem? Polki i Polacy chcą wiedzieć, czy będą pieniądze z Unii, czy otrzymamy fundusz pomocowy. A jeśli jednak zawetujecie, to co powiecie studentom, którzy nie będą mogli brać udziału w programie Erasmus+? Dacie w zamian wizy do Kazachstanu czy otworzycie staże w węgierskich laboratoriach? O ile w ogóle takie są. Ile naprawdę nas kosztuje groźba tego weta? Jakie w związku z tym wetem są i będą stosunki z innymi krajami członkowskimi? Jeśli tak, to miejcie odwagę to powiedzieć głośno i wyraźnie, bo my wam takiego prawa nie daliśmy. A jeżeli to weto doprowadzi do wyjścia z Unii, to jak będzie wyglądała rzeczywistość, transformacja energetyczna w Polsce? Za co wybudujemy infrastrukturę potrzebną do rozwoju zielonej energii? Kto nam da pieniądze? Orbánowi da Putin, mają podpisane umowy. A kto da Kaczyńskiemu? ale jaki uczciwy człowiek z Europy odważy się wam zaufać i dać pieniądze? Dzisiaj każdy Polak i każda Polka budzący się w tym kraju oddychają smogiem. Skąd weźmiecie pieniądze na walkę o czyste powietrze, jeśli nie z Unii? Wprowadzicie nowe podatki? Ale skąd weźmiecie te podatki, jeżeli wszyscy teraz plajtują? Jeżeli wyprowadzicie Polskę z Unii, to będzie gwałtowny odpływ inwestycji i odwrót inwestorów z polskiego rynku. A rolnicy, którzy nie będą mogli już żyć z dopłat? Komu sprzedadzą te płody rolne, jeżeli rynek unijny będzie dla nas zamknięty? Będziecie robili skup interwencyjny? Przez ile lat? W ramach unijnego budżetu jest 27 mld euro pomocy na odbudowę po pandemii - pomocy, nie kredytu. A skąd weźmiecie pieniądze na walkę z COVID-em? Może księża wam dadzą? No ale księża nie płacą podatków i też mają kasę od ludzi, więc jak ludzie nie będą mieli z czego płacić, to nawet księża zbiednieją. Kościoły popadną w ruinę, bo nie będzie funduszy z Unii na ich renowację. Od wielu dni żyjemy w sferze domysłów, tweetów i nieoficjalnych informacji, że Kaczyński to, Gowin tamto, a Ziobro jeszcze co innego. Wiem, że wy w takiej atmosferze czujecie się jak ryba w wodzie, uwielbiacie knuć po cichu, kraść, pomawiać, mącić (Dzwonek) i pałować. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II. Jako Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II wyrażamy stanowczy sprzeciw dotyczący karygodnych, skandalicznych i fałszywych oskarżeń wobec św. Jana Pawła II. Środowiska lewicowe i liberalne przy pomocy machiny propagandowej nieustannie od lat podkopywały autorytet Kościoła i samego św. Jana Pawła II. Obecnie przypuściły frontalny atak na największego z rodu Polaków, naszego umiłowanego ojca św. Jana Pawła II, przypisując mu tolerowanie czy wręcz współudział w tuszowaniu pedofilii wśród księży w Kościele katolickim. Fakty są zgoła odmienne, ale w tym ataku nie chodzi przecież o fakty i prawdę - chodzi o zaprowadzenie na gruzach Kościoła i naszych wartości narodowych i chrześcijańskich innego, nowego porządku wyzutego z wszelkich wartości. Pragniemy przypomnieć, że to właśnie papież Jan Paweł II był największym obrońcą moralności we wszystkich aspektach życia rodzinnego, społecznego, politycznego, również w Kościele. Papież był wielkim piewcą wolności, ale wolności, która rodzi się z prawdy, a potem wiąże się ze zobowiązaniami, wolności danej i zadanej. To on uczył nas cywilizacji miłości i życia w prawdzie, która wyzwala człowieka i czyni go w pełni wolnym. To on przeprowadził nas przez Morze Czerwone do wolnej ojczyzny. To również ojcu św. zawdzięczamy naszą wolność, którą codziennie wypełniamy treścią. Dlatego wzywam Polki i Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli: nie bądźmy bierni, stańmy odważnie w obronie naszych narodowych wartości i Kościoła. To Kościół katolicki był fundamentem naszej państwowości, a przez minione wieki był ostoją naszych wolnościowych i narodowych aspiracji. Nawet w najtrudniejszych czasach niewoli i wojen księża katoliccy krzewili polskość, nie wahali się złożyć w ofierze swojego życia. Wspomnieć należy tutaj chociażby ks. Ignacego Skorupkę, który zginął, prowadząc młodzież do ataku w wojnie z bolszewikami, czy ks. Jerzego Popiełuszkę, męczennika za prawdę i wolność, i wielu, wielu innych naszych bohaterskich kapłanów. To dziś nasz obowiązek wobec przodków, to nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! 8 grudnia wojewoda pomorski Dariusz Drelich ogłosił listę miast i wsi, które otrzymają rządowe wsparcie w ramach drugiej tury funduszu inwestycji lokalnych. Tym razem dla województwa pomorskiego zostało przyznanych 237 mln zł. Pytanie: Jaką kwotę uzyskały Gdynia, Sopot i Gdańsk? Budowa ulic, termomodernizacje, projekty prozdrowotne, przeciwpowodziowe - te wszystkie projekty odrzucono. Można odnieść wrażenie, że rząd po raz kolejny rozdaje pieniądze według przynależności politycznej i partyjnego klucza. Pokazuje, że obawy samorządowców, którzy 1 grudnia zgasili światła na znak protestu, okazały się słuszne. Panie Premierze! To pan ostatnio mówił, że trzeba skończyć z Polską A, B i C. Jednak gdy przychodzi do konkretów, to właśnie pan dzieli Polskę i Polaków. Swoją drogą to ciekawe, do jakiej Polski pan premier zakwalifikował Trójmiasto. Zerowa kwota dofinansowania lokuje Trójmiasto w Polsce Z. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle, o wygłoszenie oświadczenia. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W sierpniu tego roku złożyłem interpelację do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kolejnych niepokojących wydarzeń w Programie 3 Polskiego Radia związanych m.in. ze zwolnieniem dyrektora Kuby Strzyczkowskiego. W interpelacji tej zwróciłem uwagę na złą sytuację w Programie 3 Polskiego Radia. Napisałem, że jeszcze nie tak dawno miłośnicy Trójki żyli falą odejść z rozgłośni znakomitych dziennikarzy. Następnie po aferze z piosenką Kazika oraz zarzutach w stosunku do Marka Niedźwiedzkiego z Trójki odeszły kolejne osoby. Od stacji odcięło się też wielu polskich muzyków. Wydarzenia te wywołały falę oburzenia u ogromnej liczby fanów Trójki. Sytuację próbował ratować i uzdrowić nowy dyrektor oraz wieloletni dziennikarz Trójki Kuba Strzyczkowski, który po krótkim okresie pracy też niestety został zwolniony. Poprosiłem na końcu wicepremiera oraz ministra Piotra Glińskiego o wyjaśnienia i odpowiedź na pytania, gdzie w tym całym zamieszaniu jest miejsce dla słuchaczy Trójki, bo to przecież ich radio, oraz jakie działania zamierza podjąć, aby słuchacze Trójki tak jak dawniej wiernie chcieli Trójki słuchać. Zwróciłem też uwagę na fakt, że jeśli ktoś wypowiada swoje zdanie, a jest ono nie po myśli PiS-u, to jest niezwłocznie zwalniany. Dodałem również, że rządzący w tej kwestii nadużywają swojej władzy. W udzielonej pod koniec listopada odpowiedzi minister Gliński stwierdził, że emisja programów i audycji, kształtowanie kwestii zatrudnienia, w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze bądź współpracy z dziennikarzami, należą do wyłącznej kompetencji zarządu spółki. Jak dodał, przepisy nie przewidują możliwości ingerowania przez akcjonariusza spółki w czynności zwykłego zarządu. Minister podkreślił również, że powoływaniem i odwoływaniem zarządu zajmuje się Rada Mediów Narodowych, która jest niezależna od ministra kultury. Pan minister dodał również, że swoje stanowisko na temat ostatnich wydarzeń prezentował w sferze publicznej, a także w stosownym komunikacie na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczył również, że jako szef resortu nie został wyposażony w instrumenty prawne umożliwiające wpływanie na decyzję zarządu. Tymczasem 1 grudnia Marcin Kozłowski, dziennikarz Gazety.pl, opublikował informację, że krótko po objęciu funkcji dyrektora Kuba Strzyczkowski został zaproszony do Rady Mediów Narodowych, gdzie przedstawił swój pomysł na Program 3. W spotkaniu wzięli również udział przewodniczący rady Krzysztof Czabański oraz prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Okazało się, że główną rolę odegrał wtedy nie kto inny jak minister kultury Piotr Gliński.

Pani Marszałek! Panie premierze Gliński, z odpowiedzi na moją interpelację można by wnioskować, że pana zakres obowiązków i kompetencji nie przewiduje możliwości ingerowania w to, co dzieje się w Programie 3 Polskiego Radia. W takim razie jak to się ma do informacji przedstawionych na łamach portalu Gazeta.pl? Z informacji tych jednoznacznie wynika, że mimo że nie ma pan instrumentów wpływu na sytuację w mediach, nadużywa pan swojej władzy. Czy tak ma wyglądać nasze państwo? Ja z całą przyjemnością słucham Trójki. Bardzo proszę. Dzisiaj przez naszą Izbę przetoczyła się debata, w której niestety nie mogłem wziąć udziału, ale której z bólem uszu wysłuchałem.

Słuchaliśmy cierpliwie tyrad obrońców cenzury oburzonych wizją likwidacji tęczowej inkwizycji. Lewica wie, że może wygrać tylko przez cenzurę i tłamszenie przeciwnych poglądów, bo fałszywe idee zwyciężają tylko wtedy, kiedy skutecznie zagłuszają krytykę. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Niestety Lewica próbuje terroryzować naukę za pomocą tzw. politycznej poprawności, próbuje swoje najbardziej absurdalne twierdzenia, np. o tym, że homoseksualizm jest biologicznie prawidłowym ukierunkowaniem popędu płciowego, stroić w piórka naukowości. A ponieważ to twierdzenie oczywiście nie wytrzymuje konfrontacji z faktami, to odwołuje się do emocji, próbuje opowiadać o jakiejś nienawiści, jakiejś fobii, jakichś urażonych uczuciach. I to niestety Lewica cierpi na faktofobię, to niestety Lewica obraża się na rzeczywistość, w związku z tym lewicowi aktywiści próbują narzucić wszystkim taką atmosferę, w której po prostu nie wypada stawiać pewnych pytań, podawać pewnych faktów. To lewa strona jest tutaj agresorem i próbuje siłą powstrzymywać debatę, wyrzucając właśnie ludzi z pracy na uniwersytetach, jeśli spróbują temu się sprzeciwić. Jeśli ktoś chciałby pokazać np. w badaniach, że homoseksualizm jest po prostu niezdrowy, to prędzej zostanie zaszczuty, niż pozwoli mu się w spokoju dokończyć badania. Z drugiej strony pseudonaukowy bełkot o 72 płciach może liczyć na hojne wsparcie swoich badań z pieniędzy podatników, którym te brednie oczywiście nie są do niczego potrzebne. Na wolnym rynku nikt by takich badań nie kupił, więc Lewica zmusza nas do ich kupowania poprzez państwowe uczelnie. Ale okej, naukowcy mają prawo się mylić, prawo do błędu jest niezbędne dla postępu nauki, i dlatego tolerujemy nawet na uczelniach profesorów ekonomii, którzy twierdzą, że socjalizm działa. A wiadomo, że nie działa, rząd codziennie to sprawdza, codziennie się okazuje, że nie działa, ale mimo to są odporni na fakty akademicy. Gorzej, że z drugiej strony nie ma żadnej gotowości do debaty i Lewica uważa, że może dekretować z góry to, co jest w nauce dopuszczalne, a co nie jest.

Niestety, my też płacimy podatki na uczelnie, my, ludzie, którzy mamy inne poglądy. Skoro nie śmierdzą wam nasze podatki, skoro bierzecie je hojnie na finansowanie również swoich bełkotów, to musicie niestety zaakceptować fakt, że uczelnie to nie jest wasz folwark prywatny i że ludzie wyznający wolnorynkowe, konserwatywne wartości tak samo mają prawo je wyrażać. Nie zgadzamy się z tym, żeby za wyrażenie poglądu, że aborcja jest złem, że homoseksualizm jest zaburzeniem (Dzwonek), że kobiety różnią się od mężczyzn, ludzie byli usuwani z uczelni. To niestety studenci, którzy domagają się usuwania takich wykładowców, powinni być usuwani z uczelni, bo najwyraźniej nie rozumieją, na czym polega wolność akademicka, i z takich studentów, którzy uważają, że mają prawo zamykać usta wykładowcy, nic dobrego już nie wyrośnie, wyrosną tylko kolejni fanatycy tęczowej inkwizycji.

Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle, do wygłoszenia oświadczenia. Wysoka Izbo! Wczoraj rano na stronach internetowych urzędów wojewódzkich w całej Polsce ukazały się wyniki naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, funduszu, który miał pomóc, zgodnie z zapowiedziami, wszystkim polskim samorządom, które z jednej strony borykają się ze spadającymi w znacznym stopniu dochodami, a z drugiej strony obarczone są ogromnymi kosztami walki z epidemią. Dla województwa lubelskiego przeznaczonych zostało 313 mln zł. Natomiast samorządowcy, kiedy zobaczyli wyniki tego naboru na Lubelszczyźnie, poczuli się pokrzywdzeni.

Wsparcia finansowego nie dostał Lublin, nie dostały Puławy, Łuków, Kraśnik, Włodawa, Biłgoraj, Biała Podlaska itd., itd. Dlaczego? Dlatego, że prezydenci i burmistrzowie tych miast nie należą do Prawa i Sprawiedliwości ani z tą partią nie sympatyzują.

Na poniedziałek został zwołany Lubelski Zespół Parlamentarny, który właśnie o to szczegółowo pana wojewodę lubelskiego będzie wypytywał. Obiecuję, że żaden pokrzywdzony samorządowiec z tą krzywdą nie zostanie sam. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.